Wysoka Izbo! Wczoraj w nocy wpłynął bezprecedensowy wniosek o to, abyśmy zmienili tryb głosowania nad budżetem.

Doprowadziliście państwo do sytuacji, w której szkoła na Podkarpaciu, przedszkole w Zachodniopomorskiem, szpital w Podlaskiem i każda inwestycja w całym kraju, którą posłanki, posłowie zgłosili, mają być wrzucone do worka, który poprzecie, dlatego że jest wasz, albo odrzucicie, bo jest opozycji. Nie ma zgody na to, abyśmy poprawki do budżetu państwa traktowali jako narzędzie, dlatego że wam się nie chce po prostu dłużej pracować. Te kilkaset głosowań daje szansę na to, że ludzie z powiatów, województw i gmin będą wiedzieli, że walczymy o ich interesy, ale i dajemy szansę, żeby te poprawki przeszły. Wolicie w ciągu 10 minut załatwić sprawę, która jest interesem społecznym. Wycofajcie się z tego. Pani marszałek, ta przerwa niech będzie szansą na to, żeby Prawo i Sprawiedliwość wycofało wniosek, który dzisiaj daje szansę, że wy będziecie krótko pracowali, ale polskie gminy, polskie samorządy utracą prawo do tego, żeby mieszkańcom godnie się żyło. Po drugie. po drugie. jest to wniosek, który nie wpłynął w nocy. Po trzecie, jest to wniosek zgodny z regulaminem, panie pośle. Tak, o przerwę. Ale jeszcze pan poseł Cezary Tomczyk, Koalicja Obywatelska, wniosek formalny. Proszę bardzo. Szanowni Państwo! Zgłaszam wniosek formalny o odroczenie obrad do jutra w związku z tym haniebnym wnioskiem, który został zgłoszony przez klub PiS-u. Szanowni państwo, ja chciałem dzisiaj tylko przestrzec. Wszyscy pamiętamy rok 2016, wszyscy pamiętamy, co zrobiliście w sali kolumnowej. Wszyscy pamiętamy, jak chcieliście, żeby demokracja umarła. Na to absolutnie nie ma zgody. Dzisiaj marszałek Kuchciński siedzi tam. Ja chciałbym do pani marszałek też bezpośrednio się zwrócić i przypomnieć, gdzie marszałek Kuchciński jest dzisiaj i jak skończył po tym, co zrobiono w sali kolumnowej. Szanowni państwo, głosowanie nad budżetem, zgłaszanie poprawek to święte prawo posłów, święte prawo każdego z nas, bo nasz mandat w tej Izbie jest po prostu równy. To tak jak w domu - każdy ma prawo głosować nad poprawkami budżetowymi. I z tego miejsca chcę powiedzieć bardzo jasno: to nie jest budżet PiS-u, to jest budżet państwa. Jeżeli mamy siedzieć tutaj 30 godzin i głosować, to bardzo dobrze, bo mamy głosować nad najważniejszymi sprawami [[Oklaski]] w Polsce: w sprawie [[Dzwonek]] finansowania telewizji publicznej.

Po drugie, panie pośle, dziękuję bardzo. Chcecie uniknąć dyskusji o najważniejszej sprawie dla Polaków.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Dodatkowe sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, druki nr 828 i 828-A. Sejm na 23. posiedzeniu w dniu 16 grudnia zgodnie z art. 47 ust. 1 regulaminu Sejmu skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 836 do Komisji Finansów Publicznych w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu. Było zgłoszonych 36 poprawek. Po analizie wszystkich i po głosowaniach Komisja Finansów Publicznych wnosi do Wysokiej Izby o przyjęcie 14. poprawek i wniosków do tych punktów, a 22 rekomenduje odrzucić. Komisja przedstawia również wnioski mniejszości, a także w dodatkowym sprawozdaniu poprawki, nad którymi głosować będziemy w pierwszej kolejności. Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

441 - za, nikt nie był przeciw, wstrzymało się 11. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 1. wniosku mniejszości, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm wniosek mniejszości odrzucił.

Głosujemy.

Sejm poprawki odrzucił. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 2. wniosku mniejszości, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm wniosek mniejszości odrzucił. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 5. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 6. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm poprawkę przyjął. Głosujemy.

Sejm propozycje odrzucił. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 4. wniosku mniejszości, zechce nacisnąć

Sejm wniosek mniejszości odrzucił. Komisja wnosi o jej odrzucenie. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 13. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm poprawkę odrzucił. Komisja wnosi o ich odrzucenie.

Komisja wnosi o jej odrzucenie. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 16. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm poprawkę odrzucił. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 17. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 5. wniosku mniejszości, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm wniosek mniejszości odrzucił. Głosujemy.

Sejm poprawkę przyjął.

Głosujemy.

Sejm poprawki odrzucił. Komisja wnosi o ich przyjęcie.

Sejm poprawki przyjął. Głosujemy.

Sejm poprawkę odrzucił. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 29. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm poprawkę odrzucił. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 6. wniosku mniejszości, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm wniosek mniejszości odrzucił. Głosujemy.

Sejm poprawkę przyjął. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 31. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

409 - za, nikt nie był przeciw, wstrzymało się 46. Sejm poprawkę przyjął. Głosujemy.

455 - za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 35. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

Przystępujemy do głosowania nad całością projektu ustawy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 836, wraz z przyjętymi poprawkami, zechce nacisnąć przycisk.

439 - za, nikt nie był przeciw, wstrzymało się 17. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 5. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych o rządowym projekcie ustawy o rezerwach strategicznych (druki nr 829 i 839) - kontynuacja. Sejm na 23. posiedzeniu wysłuchał sprawozdania komisji oraz przeprowadził dyskusję, w trakcie której zgłoszono wniosek o odrzucenie projektu ustawy w całości, poprawki oraz wniosek o przystąpienie do trzeciego czytania bez odsyłania projektu ustawy do komisji. Zestawienie poprawek zostało doręczone do druku nr 839. W pierwszej kolejności przystąpimy do głosowania nad wnioskiem o przejście do trzeciego czytania projektu ustawy bez odsyłania projektu ustawy do komisji. Odrzucenie tego wniosku oznaczać będzie, że Sejm skierował projekt ustawy do Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych w celu przedstawienia dodatkowego sprawozdania. Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem o przejście do trzeciego czytania bez odsyłania projektu ustawy do komisji. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku o przystąpienie do trzeciego czytania projektu ustawy z druku nr 839 bez odsyłania do komisji, zechce nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał?

Sejm wniosek przyjął. Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy z druku nr 839. W pierwszej kolejności pod głosowanie poddam zgłoszony w drugim czytaniu wniosek o odrzucenie projektu ustawy w całości. W przypadku jego odrzucenia głosować będziemy nad zgłoszonymi poprawkami. Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem o odrzucenie projektu ustawy w całości. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku o odrzucenie w całości projektu ustawy z druku nr 839, zechce nacisnąć przycisk. się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 2. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm poprawkę odrzucił.

Sejm poprawkę odrzucił. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 4. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm poprawkę odrzucił.

Głosujemy.

Sejm poprawki odrzucił. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 839, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm uchwalił ustawę o rezerwach strategicznych. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 6. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2021 (druki nr 640, 785 i 785-A) - trzecie czytanie. Proszę pana posła Henryka Kowalczyka o przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji. Szanowna Pani Marszałek!

Ten wniosek Komisja Finansów Publicznych zaopiniowała negatywnie i rekomenduje odrzucenie tego wniosku. Zgłoszono również trzy poprawki dotyczące części tekstowej ustawy oraz 276 poprawek do załączników, czyli do części tabelarycznej. Jeśli chodzi o pracę nad tymi poprawkami, komisja wczoraj przez cały dzień pracowała nad nimi, posłowie mieli możliwość krótkiego uzasadnienia tych poprawek. W wyniku tych prac Komisja Finansów Publicznych rekomenduje przyjęcie 17 poprawek, natomiast 261 poprawek proponuje odrzucić. Warto jeszcze nawiązać do pierwszego czytania i pracy komisji w czasie pierwszego czytania projektu ustawy budżetowej, dlatego że w czasie prac komisyjnych zgłoszono 715 poprawek. Oczywiście część z nich została przyjęta, część została odrzucona, ale zdecydowaną większość odrzuconych poprawek, czyli 602 poprawki, zgłoszono jako wnioski mniejszości. Ja oczywiście odbieram to jako próbę destrukcji prac parlamentarnych, no bo po cóż zgłaszać.

skoro one były już omówione w czasie prac komisji.

Jest to wniosek o zmianę sposobu przeprowadzenia głosowania.

Zgłaszam w imieniu Koalicji Obywatelskiej wniosek przeciwny. Szanowni państwo, wprowadzacie 10 nowych podatków, 10 podatków podwyższacie. To są rzeczy, o których nie chcecie rozmawiać. Jako jedyny kraj w Europie nie chcecie zwiększać wydatków na służbę zdrowia w okresie pandemii. O tym nie chcecie rozmawiać.

to pani marszałek robi tak: te dwie kartki łączy - i ja mam głosować za tym pakietem. To jest sprzeczne z jakąkolwiek logiką, pani marszałek i szanowni państwo. A to jest nasze prawo, żebyśmy mogli [[Dzwonek]] zagłosować i wybrać poprawki, które są dla nas ważne. Jedna informacja, która jest bardzo ważna. Szanowni państwo, dwóch naszych posłów zostało wczoraj pilnie wezwanych do prokuratury w sprawie pakietów Jacka Sasina. Pani prokurator poinformowała, że przesłuchanie ma charakter pilny i polecenie przyszło z samej góry. Informuję, że złożono wniosek formalny na podstawie art. 184 ust. 3 pkt 9 regulaminu Sejmu o zmianę sposobu przeprowadzenia głosowania polegającą na głosowaniu łącznym nad poprawkami zaopiniowanymi pozytywnie przez komisję, a także łącznym głosowaniu nad poprawkami zaopiniowanymi negatywnie i wnioskami mniejszości. Uchwała Prezydium Sejmu nr 45 z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wykładni art. 184 ust. 3 pkt 9 regulaminu Sejmu brzmi następująco: „Zmiana sposobu prowadzenia głosowania może polegać także na łącznym głosowaniu poprawek w oparciu o wnioski o ich przyjęcie albo odrzucenie przedstawione przez komisje w dodatkowym sprawozdaniu, przy czym jako poprawki z wnioskiem o odrzucenie należy traktować również wnioski mniejszości zamieszczone w sprawozdaniu komisji” Oznacza to, że wniosek spełnia wymogi formalne i podlega rozstrzygnięciu przez Sejm. Przystępujemy do głosowania nad tym wnioskiem. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku formalnego o zmianę sposobu przeprowadzenia głosowania zgodnie z wykładnią zawartą w uchwale Prezydium Sejmu nr 45, zechce nacisnąć przycisk. do kogo to było? Do kogo to było?

Do wszystkich państwa kieruję tę uwagę - do wszystkich.

Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy z druku nr 785. Komisja przedstawia również wnioski mniejszości, a także w dodatkowym sprawozdaniu wniosek o odrzucenie ustawy w całości oraz poprawki. W pierwszej kolejności pod głosowanie poddam wniosek o odrzucenie projektu ustawy w całości.

Proszę usiąść, panie pośle, bardzo pana proszę. Głosujemy. Jesteśmy w trakcie głosowania.

Sejm wniosek odrzucił. Przechodzimy obecnie zgodnie z decyzją Sejmu do łącznego głosowania nad poprawkami rekomendowanymi przez komisję do przyjęcia.

Nad tymi propozycjami głosować będziemy łącznie. Głosujemy.

Konsekwencją przyjęcia niektórych poprawek będą odpowiednie zmiany w innych przepisach i załącznikach do ustawy budżetowej.

Konwent Seniorów zdecyduje, czy reasumpcja głosowania jest potrzebna. Wysoki Sejmie! W imieniu klubu Koalicji Obywatelskiej i Lewicy składam wniosek o reasumpcję głosowania. Debata budżetowa była kiedyś najważniejszą debatą w Sejmie. Dyskutowaliśmy wtedy o tym, jaka ma być Polska. Wy zniszczyliście debatę o państwie, tak jak zniszczyliście państwo. Zostały tylko wasze partyjne i prywatne interesy. W tym budżecie PiS skazuje tysiące osób chorych na raka i na choroby serca na śmierć. Ludzie będą padać jak muchy, tak jak padali w tym roku, dlatego że w czasie pandemii oszczędzacie na ochronie zdrowia. Ważniejsza jest propaganda, przekop Mierzei Wiślanej i wasze megalomańskie pomysły. Tymczasem codziennie umierają tysiące Polek i Polaków. Dziękuję. Proszę Konwent Seniorów do saloniku.

Proszę państwa, Konwent się zebrał. Chodziło o to, że jeden poseł z Koalicji Obywatelskiej nie mógł zagłosować, ale różnica głosów była tak duża, że reasumpcji nie będzie. Proszę państwa, na tym zakończyliśmy rozpatrywanie punktów porządku dziennego zaplanowanych na dzień 17 grudnia. Informuję, że zgłosili się posłowie w celu wygłoszenia oświadczeń poselskich. Proszę państwa, od razu zapowiem: czekamy jeszcze na ustawy, które przyjdą z Senatu, być może będą dzisiaj, w związku z tym potem, na końcu tego posiedzenia, będzie ogłoszona przerwa do dziś do godz. 19. Ewentualnie, jeżeli nie przyjdą te ustawy, to będziemy tę przerwę przesuwać, dobrze?

Wysoka Izbo! 39 lat temu miała miejsce krwawa pacyfikacja protestu w Kopalni Węgla Kamiennego Wujek w Katowicach. Protest górników był gestem wsparcia dla aresztowanego Jana Ludwiczaka, przewodniczącego „Solidarności” w kopalni. Protest rozpoczął się 14 grudnia. Zapanowanie nad górnikami miało strategiczne znaczenie dla komunistycznych władz, od tego uzależniono powodzenie wprowadzonego stanu wojennego. Decyzję o użyciu siły podjęto 15 grudnia, podczas narady wojewódzkiego komitetu obrony. Do kopalni skierowano prawie 1500 funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej i ZOMO oraz 760 żołnierzy dysponujących 22 czołgami i 44 wozami bojowymi.

Trzech zmarło w wyniku odniesionych ran. Pacyfikacja pokazała prawdziwe oblicze komunistów, a jej brutalny charakter spowodował, że działacze opozycji, którzy nie zostali internowani na początku stanu wojennego, zmienili koncepcję walki z reżimem. Na premedytację ówczesnej władzy jednoznacznie wskazuje charakter ran postrzałowych: jama brzuszna, czaszka, klatka piersiowa. W wyniku pacyfikacji zginęło dziewięciu górników, a 20 zostało rannych. Ani Wojciech Jaruzelski, stojący na czele Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, ani Czesław Kiszczak nie zostali pociągnięci do odpowiedzialności. Ukarano jedynie Romualda Cieślaka, dowódcę plutonu specjalnego ZOMO, który dostał karę 6 lat pozbawienia wolności, wraz z kilkunastoma jego podwładnymi - kary 3 lat pozbawienia wolności. Pacyfikacja kopalni Wujek nazywana jest największą zbrodnią stanu wojennego. Proszę bardzo.

Pani Marszałek! Rozpoczyna się adwent, a mnie przypominają się wielkopostne obrazy ewangeliczne. Oto do Jerozolimy wjeżdża na osiołku Jezus, witają go wiwatujące tłumy. Są jego nauki, cuda, może ktoś dyskretnie dotknie jego szaty. Już z własnego doświadczenia pamiętam przyjazdy Jana Pawła II Wielkiego do ojczyzny. Był radosny śpiew, rzesza ludzi zasłuchanych w jego słowa, świętowanie, wzruszenia, wielkie przeżycia. I dzień jego odejścia do domu Ojca, nocne czuwania w kościołach, łzy i muzyka dzwonów. Przecież to tak niedawno, a już słychać wołania: winien jest!

Skąd niszczenie wystaw, pomników, nazw ulic? I tak niewiele głosów obrony, a przecież Wielki jest. Pięciomilionowy tłum wołał na placu św. Piotra: święty od zaraz, natychmiast święty! Może by jakiś Piłat przynajmniej umył ręce i stwierdził publicznie: nie znajduję w nim żadnej winy. Smutno, ale wierzę, że obudzi się nam ojczyzna, że będzie jeszcze u nas, jak należy, choć tych bolesnych porównań może być znacznie więcej. Popatrzmy na wieś i miasto. Podobno socjologowie odkryli, że młodzi Polacy osiedlający się w mieście wstydzą się swoich wiejskich korzeni. Smutni outsiderzy, ale to nie ich wina. Ucieczka od własnego dzieciństwa jest bolesna tak jak utrata domu, ale nie każdy ma dość odwagi, aby przeciwstawić się drwinom wypowiadanym pod adresem jego przodków. Kiedyś to wieś dostarczała wzorców kulturowych, szlachecki dwór był wzorem polskiego domu, a do bohaterstwa, do heroizmu nawet nie trzeba było nikogo przekonywać, bo to była sprawa honoru. Tak naprawdę nie jest ważne, gdzie ogląda się wschody i zachody słońca, tylko czy się zauważa ich piękno. Ważne jest, czy chce się być człowiekiem prawdziwym, a ludzie wsi wiedzą, że więcej jest tych, którzy swoją wieś i swój wiejski rodowód kochają, niż tych, którzy chcą być uciekinierami od własnej kultury. Problem podziału na wieś i miasto jest sztuczny i wywoływany po to, aby ludzi dzielić, skłócać, budzić niechęć czy wpędzać w kompleksy. Może wtedy łatwiej przekonać, że dziś nie wolność, ale pieniądze bardziej się liczą, nie człowieczeństwo, mądrość, wiara i rozum (Dzwonek), wierność i odpowiedzialność, ale jakieś ideologiczne fanaberie wydumane na brukselskim bruku. Słowo „adwent” pochodzi z łaciny i tłumaczy się je jako oczekiwanie. Tegoroczny adwent jest nabrzmiały od problemów, więc i oczekiwań jest wiele. Najważniejsze jest jednak to, aby żyjąc, jak trzeba, nie zniszczyć wartości nadchodzących świąt. Jeśli odbierze się ludziom niedziele, czas na refleksję, odpoczynek i świętowanie, czym będą święta? Narodzi się Chrystus czy kolejny raz go ukrzyżujemy? Będziemy śpiewać polskie kolędy czy słuchać złowrogich wrzasków, niezrozumiałych i niczym nieuzasadnionych? We Francji młodzi katolicy wyszli na ulice, aby domagać się otwarcia kościołów. Chcą się modlić. To dobry znak. Pozwala wierzyć, że na folwark wróci człowiek. To tylko kwestia czasu - tak mówią wizjonerzy i mają rację. Świat bez człowieka żyjącego prawdą jest jak zniszczony przez szkodnika las - smutny, pozbawiony Bożego uśmiechu. Dziękuję, panie pośle. Bardzo proszę, pan poseł Paweł Rychlik, Prawo i Sprawiedliwość. Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

Wysoka Izbo! Wczoraj minęła 39. rocznica tragedii w kopalni Wujek, w której śmierć poniosło dziewięciu górników, a dziesiątki, często nieokreślonych, zostało rannych. Kopalnia Wujek stała się symbolem heroizmu, dążenia do wolności ojczyzny, walki o godność i prawa człowieka. Dzisiaj należy oddać hołd bohaterom tamtych ciemnych, grudniowych dni. Łączymy się w modlitwie i w zadumie z rodzinami ofiar zamordowanych górników, z więzionymi i internowanymi w stanie wojennym górnikami kopalni Wujek, członkami śląsko-dąbrowskiej „Solidarności”, jak i w całej Polsce. Nazwiska górników poległych za wolność ojczyzny muszą pozostać symbolem walki o suwerenność naszej ukochanej ojczyzny.

Nigdzie jak właśnie w Wujku nie było tak oczywiste, że komuniści wypowiedzieli wojnę własnemu narodowi i że odpowiedzialni są za to gen. Jaruzelski i gen. Kiszczak. Dzisiaj, w kolejną rocznicę wydarzeń w kopalni Wujek, jeszcze raz składamy hołd bohaterom tamtych wydarzeń, bohaterom stanu wojennego. Składamy wyrazy szacunku i wszyscy chylimy czoło przed wszystkimi internowanymi, więzionymi, dzięki którym dzisiaj mogę przemawiać w Wysokiej Izbie. Dziękuję.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Chciałbym zwrócić szczególną uwagę na niebezpieczną sytuację, jaka panuje w mieście Morąg, a jest ona związana z kładką nad torami kolejowymi. Jest to w województwie warmińsko-mazurskim. W kwietniu br. od konstrukcji kładki odpadł element metalowy, kątownik metalowy o długości ok. 1 m, który upadł na czynny peron, z którego korzystają podróżni. Na szczęście nikt nie ucierpiał, bo w tym czasie peron był pusty.

Do dnia dzisiejszego wspomniane przejście jest niedostępne dla pieszych. Jest to poważny kłopot dla mieszkańców Morąga, bowiem uniemożliwia to sprawne przedostanie się z jednej części miasta do drugiej części. Zamknięta kładka w znaczący sposób utrudnia morążanom codzienne życie. W związku z licznymi sygnałami otrzymywanymi od moich wyborców 7 grudnia spotkałem się z burmistrzem miasta Morąga panem Tadeuszem Sobierajskim. Pan burmistrz wyraża chęć współpracy w sprawie remontu przejścia i zobowiązał się również w piśmie, które skierował do PKP SA Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku, do partycypacji w kosztach remontu. Problem, który uniemożliwia rozpoczęcie prac remontowych, to ustalenie właściciela kładki. Zdaniem burmistrza Morąga to PKP SA jest właścicielem obiektu. Zgodnie z decyzją wojewody warmińsko-mazurskiego z dnia 12 marca 2004 r. właścicielem kładki jest spółka SA.

Pani Marszałek! Chciałbym zwrócić szczególną uwagę i przede wszystkim zwrócić się do ministra infrastruktury oraz do ministra aktywów państwowych o pilne ustalenie właściciela kładki nad torami w Morągu oraz jak najszybszy jej remont, bo stan kładki zagraża bezpieczeństwu podróżnych.